Wysoka Izbo! Chcę złożyć wniosek formalny w celu zwołania Konwentu Seniorów, w czasie przerwy oczywiście, w celu uzupełnienia porządku obrad o wniosek o zbadanie odpowiedzialności poszczególnych członków rządu za zbędne bądź nadmierne doprowadzenie do paraliżu życia społecznego, a także polskiej gospodarki, i być może powołania w tym celu komisji śledczej. Proszę państwa, rozumiem, że wszyscy imitowaliśmy pewną zarazę, która szła z Zachodu, ale pozostaje zbadać np., czy niewiara w to, że ludzie sami potrafią założyć maseczki. Czy przypadkiem nakaz nie jest powodowany tym, że ktoś chciał zrobić interes na sprowadzaniu maseczek itp. rzeczy. Konwentu nie zwołam, panie pośle, bo to moje uprawnienie. Został zgłoszony wniosek formalny o przerwę. Poddam ten wniosek pod głosowanie. Kto z pań i panów posłów jest za zarządzeniem przerwy?

Sejm wniosek odrzucił. Wniosek formalny, pan poseł Krzysztof Gawkowski, Lewica. Proszę. Wysoka Izbo! Wczoraj klub koalicyjny Lewicy zgłosił projekt ustawy o abolicji mandatowej.

Kilka tygodniu temu tutaj, w Izbie, mówiliśmy, że trzeba nakładać mandaty. Prawo i Sprawiedliwość, wnioskodawcy mówili, że będziemy nakładali mandaty na osoby bez masek, ale mandaty te zostały nałożone tylko na tych, którzy nie mieli legitymacji Prawa i Sprawiedliwości. 15 mln zł z mandatów ma dzisiaj pokrywać koszty budżetowe. To są ludzie, którzy nie mają pieniędzy, a którzy zostali często niesłusznie ukarani. To jest ustawa, która ma pokazać sprawiedliwość ponad podziałami politycznymi. Zwracam się z wnioskiem formalnym i ponawiam prośbę: bądźmy posłami równymi obywatelom, a nie posłami ponad obywatelami.

Szanowna Pani Marszałek! Chciałbym prosić panią marszałek o zmianę sposobu prowadzenia obrad, skorzystanie z prawa, które pani marszałek posiada, i dopuszczenie w tej debacie do zadawania pytań.

Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy pracowali podobnie, tzn. może nie 30 czy 25 dni. Chodzi o to, żebyśmy każdą z tych poprawek, którą przedstawił nam Senat, po prostu przedstawili. Tak się w Sejmie pracowało zawsze. Warto do tego wrócić. Jeśli pan poseł Czarnek w Senacie zobaczył, że to jest możliwe, mówił o porozumieniu, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby podobnie było w Sejmie.

Dziękuję, panie pośle. Panie pośle, chciałabym na jedno zwrócić uwagę. Natomiast mogą być pytania. Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tej uchwały. Proponuję, na podstawie art. 54 ust. 8 regulaminu Sejmu, rozpatrzenie uchwały bez uprzedniego skierowania jej do komisji. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 16. porządku dziennego: Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (druk nr 399) Przypominam, że Sejm odrzuca poprawki Senatu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeżeli Sejm nie odrzuci poprawki Senatu, uważa się ją za przyjętą. W punktach porządku dziennego dotyczących rozpatrywania poprawek Senatu głosować będziemy nad wnioskami o odrzucenie poprawek Senatu. W 1. poprawce do art. 3 ust. 1 pkt 1 Senat proponuje m.in. zmianę terminu zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego dla wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Panie pośle, bardzo proszę.

Dziękuję, panie pośle. Wnioskodawca, pan poseł Przemysław Czarnek. Proszę bardzo. Ta poprawka przede wszystkim doprecyzowuje tylko jedną rzecz, mianowicie że zgłosić się można do głosowania korespondencyjnego w gminie, w której się jest umieszczonym w spisie wyborców.

Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 1. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Pan poseł Robert Kropiwnicki, Koalicja Obywatelska, pytanie. Proszę bardzo, pani poseł Fabisiak. Nieprzyjęcie tej poprawki wykluczy możliwość głosowania całej Polonii, bowiem dotychczasowy zapis mówiący o tym, że konsulat musi na 6 dni przed wyborami dostarczyć karty do głosowania, uniemożliwia właściwie wszystkim wzięcie udziału w głosowaniu, bo przecież mamy wiele takich listów.

Zatem ta poprawka jest niezbędna dla tych 60, 100 czy 200 tys. ludzi, przedstawicieli Polonii, którzy uczestniczą w wyborach, a którzy będą to mieli uniemożliwione, jeśli poprawka Senatu nie zostanie przyjęta. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 2. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów.

Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 3. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 4. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Za - 3, 451 - przeciw, nikt się wstrzymał. Sejm poprawkę Senatu przyjął. W 5. poprawce do art. 3 ust. 6 Senat proponuje, aby w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego niepełnosprawny wyborca głosujący w kraju mógł żądać także dostarczenia pakietu wyborczego do drzwi lokalu, którego adres został wskazany w zgłoszeniu. Proponuję, aby Sejm wyraził zgodę na łączne głosowanie nad poprawkami 5., 7. i 16. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Pytanie, pani poseł Wanda Nowicka. Proszę bardzo. Wysoka Izbo!

Kto wie, jaka jest skala problemu, ile osób będzie potrzebowało skorzystania z takiej możliwości? W jaki sposób zagwarantujemy, że do wszystkich zainteresowanych osób niewidomych bądź niedowidzących dotrze informacja, że mogą skorzystać ze swojego prawa wyborczego? Dziękuję bardzo. Poproszę pana posła Przemysława Czarnka. Wysoka Izbo! Wyraziłem radość z tego, że przynajmniej część senatorów opozycji w Senacie, czy tej większości senackiej. potrafiła wznieść się ponad podziały polityczne i pracować merytorycznie nad tym, co zaproponowaliśmy. To mnie cieszyło, a nie sposób procedowania.

Niestety taka jest sytuacja.

Również osoby niewidome będą mogły zorientować się, że mają uprawnienie do tego, żeby tej nakładki żądać. Dziękuję bardzo.

Nikt nie był za, 453 - przeciw, nikt się nie wstrzymał. Sejm poprawki Senatu przyjął.

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 8. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Proponuję, aby Sejm wyraził zgodę na łączne głosowanie nad poprawkami 9. i 14. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek 9. i 14., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

1 - za, 451 - przeciw, nikt się nie wstrzymał. Sejm przyjął poprawki Senatu. Proponuję, aby Sejm wyraził zgodę na łączne głosowanie nad tymi poprawkami. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę.

Kto jest przeciw?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął. W 11. poprawce do art. 8 ust. 1 i 2 Senat proponuje m.in. zmiany w zakresie treści wpisywanych przez wyborcę na kopercie zwrotnej. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 11. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

2 - za, 451 - przeciw, nikt się nie wstrzymał. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. W 12. poprawce do art. 8 Senat proponuje, aby dodać ust. 2a doprecyzowujący zasady głosowania korespondencyjnego przez wyborcę podlegającego obowiązkowej kwarantannie lub izolacji.

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Senat proponuje określenie zasad instalacji dodatkowych nadawczych skrzynek pocztowych. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 13. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 15. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów.

Proszę bardzo. Pani Marszałek! Polki i Polacy zasługują na prawdę, zasługują na normalną możliwość dowiedzenia się, jak wyglądają nasi kandydaci, jakie są programy, zasługują na informację pozbawioną propagandy politycznej i zasługują też na informację, która będzie mogła prezentować w pełni, wyraźnie i spokojnie programy kandydackie. My serdecznie namawiamy do wydłużenia tego czasu antenowego. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Wysoka Izbo! Boimy się o was, bo widzimy strach w waszych oczach. To jest rzeczywiście wyjątkowy kraj, jedyny taki na świecie, gdzie główne ugrupowanie opozycyjne w tych samych wyborach tego samego roku. ma dwóch kandydatów, z czego jeden ma zebrane podpisy, drugi nie ma zebranych podpisów, i jeszcze nie wiadomo, który z nich będzie kandydował. Dlatego chcecie wydłużenia czasu antenowego w mediach publicznych, żebyście się w końcu mogli zdecydować, czy pani Kidawa-Błońska, czy Trzaskowski, a może jeszcze ewentualnie marszałek Grodzki. pań i panów posłów jest za odrzuceniem 19. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

W 20. poprawce w dodawanym art. 14a Senat proponuje uregulować zbieranie podpisów poparcia dla kandydatów za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Proszę. Wysoka Izbo! Jest niezwykle istotna szczególnie w obecnych czasach. Zakłada ona możliwość zbierania podpisów poparcia dla kandydatów poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej, ePUAP. Jest to ważne z kilku względów. Po pierwsze, ze względów zdrowotnych, ponieważ zbiórka podpisów w obecnych czasach będzie mocno utrudniona. Po drugie, zbiórka podpisów zostanie usprawniona, ponieważ będzie można szybciej weryfikować te podpisy i ułatwi to pracę Państwowej Komisji Wyborczej za to odpowiedzialnej.

Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 20. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

W 21. poprawce do art. 15 ust. 1 Senat proponuje, aby czynności, o których mowa w tym przepisie, marszałek Sejmu podejmował w porozumieniu z Państwową Komisją Wyborczą. Proszę. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Otóż chodzi o to, żeby pani marszałek kalendarz czynności wyborczych i terminy tych czynności wyborczych ustaliła w porozumieniu z Państwową Komisją Wyborczą, a nie po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej.

Ta poprawka, pani marszałek, łączy się ściśle z poprawką 26., która dotyczy tego, że to minister zdrowia może, w drodze rozporządzenia, określić te gminy, w których wybory zostaną przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego.

Chciałam tylko pana uspokoić, że naprawdę od początku porozumiewam się z Państwową Komisją Wyborczą, podobnie jak Senat. A więc proszę się nie obawiać, że będę robiła coś przy negatywnej opinii Państwowej Komisji Wyborczej.

Pan poseł Krzysztof Śmiszek, Lewica. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dzisiaj już ostatni raz chyba dyskutujemy nad rolą Państwowej Komisji Wyborczej przy okazji tych wyborów prezydenckich. Chciałbym zapytać przedstawiciela wnioskodawców. Ostatni raz już mamy szansę rozmawiać w ten sposób. Proszę powiedzieć szczerze Polkom i Polakom, co tak naprawdę stoi za proponowanym przez was podpisem i czemu prawdopodobnie - widzę to już po minach posłów i posłanek Prawa i Sprawiedliwości - będziecie głosować przeciwko poprawce Senatu. A więc chciałbym zapytać: Jak to jest, że tak łatwo pozbywacie się wiodącej roli Państwowej Komisji Wyborczej?

W porozumieniu. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Zaprzeczacie sami sobie, choć akurat nie pan poseł Śmiszek, bo on nie uchwalał Kodeksu wyborczego. Sformułowanie: zaopiniowanie przez Państwową Komisję Wyborczą jest sformułowaniem kodeksowym. Ta współpraca układa się znakomicie i nie ma się czego bać, panie pośle. Myślę, że będzie niejedno pytanie.

Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 21. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

W 23. poprawce do art. 15 ust. 1 Senat proponuje, aby termin na zgłoszenie kandydata na prezydenta nie mógł upłynąć wcześniej niż w 10. dniu po opublikowaniu postanowienia o zarządzeniu wyborów. Proszę. Otóż jesteśmy w szczególnym momencie i wszyscy to wiemy. Pani marszałek dostała bardzo szerokie uprawnienia dotyczące ustalania czynności wyborczych. Chcielibyśmy bardzo pani wierzyć, ale najbardziej pani wierzylibyśmy, gdyby pani ten kalendarz po prostu opublikowała. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pani powiedziała, że będzie tyle i tyle dni na poszczególne czynności. Wyborcy Rafała Trzaskowskiego chcą wiedzieć, ile będą mieli czasu na zbieranie podpisów. Ta poprawka mówi wyraźnie, że czas na zbieranie podpisów powinien być wpisany do kalendarza, bo tak też mówi konstytucja. Art. 127 ust. 7 mówi wyraźnie: zasady i tryb zgłaszania kandydatów określa ustawa, a nie postanowienie marszałka. Tak więc przepis zgłaszany w tej poprawce Senatu jest jak najbardziej wypełnieniem dyspozycji konstytucyjnej.

Proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Wiem to, szanowny panie pośle, i dokładnie to określa nasza ustawa.

Od 13 maja prawie 20 dni trzymaliście ją w Senacie.

Gdybyście państwo tę ustawę uchwalili 2 tygodnie temu, mielibyście nie 10 dni na zbieranie podpisów, a nawet 20 dni, ale państwo tego nie chcieliście. Próbowaliście wyrzucić te wybory na jesień, bo się ich ewidentnie boicie teraz, w czerwcu. Na szczęście wycofaliście się z tego chaosu i dlatego nie będziecie mieli 1 dnia czy 2 dni na zbieranie podpisów, tylko tak naprawdę kilka. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 23. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Senat proponuje, aby uchwałę, o której mowa w tym przepisie, Sąd Najwyższy podejmował w ciągu 16 dni od dnia podania wyniku wyborów do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą. Pan poseł Marcin Kierwiński, Koalicja Obywatelska, pytanie. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Odrzucając trzy ostatnie poprawki, pokazaliście tak naprawdę, zwracam się do większości sejmowej, o co wam chodzi. Wy nie chcecie równych wyborów, wy nie chcecie równych szans. Wy chcecie cały czas manipulować przy tych wyborach, cały czas ograniczać kandydatom opozycyjnym możliwość prowadzenia kampanii wyborczej. Piękne słowa, jak pan tutaj zaklinał, ile będziemy mieli czasu, ale odrzucając tamtą poprawkę, pokazaliście jedną wielką rzecz: pokazaliście gigantyczny strach. Boicie się Rafała Trzaskowskiego. Ha, ha, ha! ...bo boicie się, że on odeśle waszego prezydenta z Pałacu Prezydenckiego, [[Oklaski]] że ta biała flaga wreszcie zniknie. Bardzo się tego boicie. Pan się teraz śmieje, ale ja muszę powiedzieć: będzie pan płakał jeszcze z tego powodu, będzie pan płakał z tego powodu.

Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 24. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Senat proponuje, aby zmiana terminu wykonania czynności wyborczych nie mogła dotyczyć terminu na zgłoszenie kandydata na prezydenta. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Wystarczyło tylko dopuścić pytania, a zwłaszcza odpowiedzi posła wnioskodawcy i dowiadujemy się bardzo ciekawych rzeczy. Na początku dowiedzieliśmy się, że niewidomi i niedowidzący będą mogli natychmiast przeczytać sobie Dziennik Ustaw zaraz po jego opublikowaniu i stąd dowiedzą się, jakie mają prawa wyborcze. Po drugie, trzeba się w końcu zdecydować, co jest merytoryczną pracą, a co jest obstrukcją.

Jednocześnie mówił o tym, że w Sejmie merytorycznej pracy nie było. No, chyba waszej pracy, wnioskodawców, bo w jednym dniu były trzy czytania, bez debaty rzetelnej. Czyli wasi posłowie wnioskodawcy, którzy w zaciszu gabinetu smażyli tę ustawę, nie wykonali merytorycznej pracy.

W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 25. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów Sejm poprawkę przyjął.

Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Pytanie, pan poseł Sławomir Nitras, Koalicja Obywatelska. Proszę. Pani Marszałek! To jest chyba jedna z najistotniejszych poprawek. Rzeczywiście jest tak, jak mówił poseł Czarnek, że w Senacie udało się w pewnych sprawach wypracować porozumienie. Wydaje się, że to, co przyjął Sejm, czyli regulacja, która pozwala wpływać na tryb wyborczy jednemu politykowi - ja tutaj abstrahuję od pana ministra Szumowskiego i jego bieżących problemów, to nie o to chodzi, ale jeden polityk swoją decyzją może kształtować tryb wyborów - to nie jest najlepszy pomysł. To, co zaproponował Senat, pozwala zainicjować ministrowi zdrowia ten proces, ale pozostawia go w rękach Państwowej Komisji Wyborczej. Apeluję do większości parlamentarnej o to, żebyście poważnie rozpatrzyli tę poprawkę i ją przyjęli. Jeżeli to zostanie w Państwowej Komisji Wyborczej i jeżeli jeszcze pani marszałek będzie tak miła i dzisiaj na tej sali przy okazji procedowania poda najważniejsze terminy, tzn. na kiedy ma zamiar ogłosić wybory.

Wysoka Izbo! Mogę? To ja od nowa. Wysoka Izbo! Przy okazji procedowania nad tą poprawką musimy się zastanowić nad tym, czy pan minister Szumowski będzie miał dobre dni czy złe dni. Jak miał dobry dzień, to powiedział, że te maseczki to tak w sumie w niczym nie pomagają, ale jak miał zły dzień, to kazał wszystkim Polakom te maseczki nosić. Jak miał dobry dzień, to pozwolił nam już iść na spacer do lasu, a gdy miał zły dzień, to powiedział, że po lasach nie wolno chodzić, bo tam to są te zarazki.

Tak więc będziecie musieli się państwo zastanowić nad tym, czy pan minister Szumowski będzie miał złe czy dobre dni, ponieważ to on będzie wydawał taką rekomendację. Moje podstawowe pytanie brzmi: Po pierwsze, czy ta rekomendacja ministra [[Dzwonek]] musi być wykonana? Ostatnie pytanie, zanim udzielę głosu panu posłowi wnioskodawcy, zada pan poseł Krzysztof Śmiszek, Lewica. Proszę bardzo. Wysoka Izbo!

Wrocław, Szczecin, Gorzów, Poznań? Wszystkie te, które są progresywne, proeuropejskie i nie głosują na PiS.

Pan poseł Przemysław Czarnek udziela odpowiedzi. Tam minister zdrowia ma absolutnie cały czas dobry humor. Więc módlmy się o to, żeby pan minister Szumowski miał cały czas zły humor, to wtedy rzeczywiście Polacy będą bezpiecznie mogli chodzić po drogach, nie zarażając się koronawirusem, tak jak to jest teraz w Polsce. A pan poseł Śmiszek, szanowni państwo. Panie Pośle!

Pan chce im zabronić głosowania korespondencyjnego?

Panie i Panowie Posłowie! Pani Marszałek! Dlatego wydaje się dość logiczne, że jeżeli nakładamy na samorządy obowiązek zapewnienia środków ochrony w siedzibach komisji, to powinno być to jednak zadanie zlecone, co oznacza, że za tym również powinno pójść finansowanie.

Dlatego chciałam spytać, czy rozważaliście możliwość sfinansowania środków ochrony dla gmin. Dziękuję, pani poseł. Pan poseł Czarnek. Proszę bardzo. Krótko: to jest oczywiste, że gminy nie mogą brać na siebie tego ciężaru. Ministerstwo Zdrowia wyposaży w konieczne środki ochrony osobistej wszystkich członków obwodowych komisji wyborczych.

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Przystępujemy do głosowania.

1 - za, 455 - przeciw, nikt się nie wstrzymał. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Pytanie zada pan poseł Konrad Frysztak, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Zwracam uwagę na słuszność tej poprawki. To byłby absolutny błąd.

Druga rzecz, szanowni państwo, to dobra poprawka Senatu wskazująca na możliwość umiejscowienia tzw. pracownika samorządowego delegowanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta. Dziś niejednokrotnie obwodowe komisje mieszczące się w szkołach mają problem.

Proszę bardzo. Wysoka Izbo! Poprawka 30., która zwiększa minimalny skład komisji wyborczych z trzech do pięciu osób, jest niezwykle zasadna.

Po drugie, tak ograniczony skład nie daje gwarancji dobrego przeprowadzenia tych wyborów. O co wam tak naprawdę chodzi?

Proszę pana posła Czarnka o udzielenie odpowiedzi na to pytanie. Pani poseł.

Pani Marszałek! Używając słów filmowego Pawlaka: No po jakiemu oni mówią, no? Później się pan poprawił pod wpływem naszej reakcji, że to jednak minimalna liczba. Otóż liczba kandydatów do obwodowych komisji wyborczych zgłoszonych przez komitet Andrzeja Dudy to 34 tys.

A jeśli zgłosicie kandydatów - nie wiem, czy pani Małgorzata Kidawa-Błońska, czy Trzaskowski, czy Grodzki - wtedy rzeczywiście będą to pełne składy komisji. Przystępujemy do głosowania. Panie Pośle!

Macie z tym problem i nie potraficie stworzyć dobrego prawa, ale proszę Jest pan posłem sprawozdawcą, chce pan rozmawiać o polityce, to proszę zabierać głos w pytaniach. Pan odpowiada za jakość ustawy i za tłumaczenie punktów.

Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 30. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Senat proponuje zmianę w procedurze łączenia obwodów głosowania. Proszę. Wysoka Izbo! Co do zasady organizacja demokratycznych, konstytucyjnych wyborów powinna być w rękach odpolitycznionej PKW i samorządów. Tymczasem państwo upolityliczniś... upo. wszystkie organy, które decydują i współdecydują o wyborach, do maksimum, a w sejmowej wersji dzisiejszego projektu wybory były wręcz w rękach ministra zdrowia wraz, z całym szacunkiem, z panią marszałek. Senatu to dobra poprawka, bo włącza na powrót do współdecydowania, np. o połączeniu obwodów wyborczych, samorząd, w tym wypadku wójtów.

Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 31. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

To jest poprawka, która mówi o protokołach obwodowych komisji wyborczych. Ta ustawa wyklucza zapisy Kodeksu wyborczego, które mówią o opieczętowaniu kart wyborczych pieczęciami Państwowej Komisji Wyborczej i obwodowej komisji wyborczej. Jeżeli karta nie jest opieczętowana, ktoś może dorzucić karty. Te pieczątki są dowodem na to, że to są karty prawdziwe.

Bardzo proszę, pan poseł Przemysław Czarnek. Bardzo za nie dziękuję. Odpowiedź też się zdarzy. Słusznie pan poseł zauważył, ale to jest pytanie do Państwowej Komisji Wyborczej, którą państwo tutaj też słusznie wychwalaliście jako tę, która świetnie przeprowadzi wybory, i tak będzie.

Chciałbym również móc docenić jakość pana odpowiedzi.

Panie Pośle! Jeszcze raz udzielam merytorycznej odpowiedzi.

Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 32. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

1 - za, 451 - przeciw, nikt się nie wstrzymał. Wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów Sejm poprawkę przyjął. W 33. poprawce do art. 20 Senat proponuje dopuszczenie możliwości przeprowadzenia szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych w formie innej niż zdalna. Pan poseł Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska, pytanie. Proszę.

Jak wszyscy wiemy, to był sprzęt wyjątkowo drogi, ponieważ przyłbice były kupowane za 48 zł, mówię o tym koncernie narciarsko-oscypkowym.

Chciałbym mieć tę pewność, że te drogie przyłbice nie zostaną dostarczone komisji wyborczej.

Panie pośle, doskonale pan o tym wie.

Proszę bardzo. Szczęść Boże! Czcigodna Pani Marszałek!

Pytanie jest, rzecz jasna, takie: Kiedy z tym skończycie?

Korzystam z okazji, by naród, naszych wyborców zachęcić do zainteresowania obywatelskim ruchem Pilnuj Wyborów. Proszę wejść na stronę, proszę ściągnąć aplikację, proszę pilnować tych wyborów, bo procedura żółwim tempem, ale wreszcie dociera do mety.

Nikt nie był za, przeciw - 450, nikt się nie wstrzymał. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął.

Proszę. Pani Marszałek! Ta ustawa jest przyznaniem się do wielkiej porażki waszego środowiska. Sprowadziliście na Polskę największy kryzys konstytucyjny ostatnich 30 lat. Nie było takiego dramatu. Kto za to odpowiada? Zdecydujcie się, czy sam prezes, czy prezes z Gowinem i panem Ziobrą, czy nieudolny Sasin, czy Koalicja Obywatelska. Sami nie wiecie kto. Powiem wam, kto za to odpowiada. Wy. Wasza nieudolność. Dlatego jesteśmy w tak tragicznym miejscu. Swoją nieudolnością spowodowaliście, że nie wiemy, kiedy będą wybory. Mamy dość takiej władzy. Mamy dość tego bałaganu. Mamy dość waszych afer. Chcemy uczciwych wyborów, bo wybory są dla Polaków, żeby wybrali uczciwego prezydenta, żeby wybrali prezydenta, któremu ufają, a nie, żeby realizować wasze sztuczki polityczne. Wy wszystko chcecie załatwiać przy zielonym stoliku. Mamy dość takiej władzy. Dobrze? Proszę państwa, zwracam uwagę: to są pytania, to jest ostatnia poprawka. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! W przeciwieństwie do kolegi posła, Lewica się cieszy, że dochodzimy do końca. Bardzo się cieszymy, że dochodzimy do końca tego procesu legislacyjnego, bo ileż można rozmawiać o wyborach, które ośmieszyliśmy 10 maja. Nie wiem, czy pan prezes Kaczyński wie, ale chciałem poinformować go, co dzieje się w Pałacu Prezydenckim, w tym większym pałacu, co tam dzisiaj opowiadają. Jak będziemy taką drogą maszerowali, to niedługo w każdym domu będzie sakwa złota, a później 100 mln. Pan prezes wie, jak to się kończy, jak się 100 mln ogłasza. Pani Marszałek! Pytanie, bo prosiła pani o pytanie. Zwracam się z apelem do pani marszałek, żeby najpóźniej w dniu jutrzejszym cała Polska poznała, kiedy mają być wybory i jaki jest kalendarz wyborczy. Panie pośle, pan doskonale wie, kiedy mogę ogłosić wybory, więc proszę tak się nie ekscytować. Jeszcze ustawy nie przyjęliśmy, jeszcze nie jest ona podpisana przez pana prezydenta, nie jest opublikowana w Dzienniku Ustaw, nie jest zaopiniowana przez PKW. więc, panie pośle, jeszcze chwila cierpliwości. Ostatnie pytanie. Proszę bardzo, ostatnie pytanie przed ostatnim głosowaniem, pan poseł Braun. Mam nadzieję, że tym razem będzie to pytanie. Kontynuując przerwany wątek, setki takich właśnie kartek rozłożono na naszych fotelach.

Pilnujcie, nie śpijcie, żeby was nie ukradli, szanowni rodacy, bo tutaj wprawdzie raz na jakiś czas zawiązuje się jakiś sojusz ponad podziałami, sojusz ponad korytami.

Minął czas. Pan poseł Czarnek.

Pani Marszałek! Wiem, że pan poseł Kropiwnicki jest z tej frakcji Schetyny, która nie popiera Budki, w związku z powyższym nie popiera Trzaskowskiego, ale mógłby pan posłuchać jednak kandydata na kandydata, który w pierwszym swoim przemówieniu. na konferencji prasowej powiedział wprost: To my - mówił - samorządowcy z Warszawy, z Poznania, nie dopuściliśmy do głosowania 10 maja.

Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 34. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie punktów porządku dziennego zaplanowanych na dzień 2 czerwca br.